Wznawiam obrady. Proszę zatem o naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu.

Obecnych jest 439 posłów. Stwierdzam kworum. Informuję, że Senat przyjął bez poprawek ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. W związku z tym planowany punkt 12. porządku dziennego stał się bezprzedmiotowy. Z wnioskiem formalnym pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Pani Marszałek! Ktoś to jednak musi powiedzieć, że moglibyście państwo robić to inaczej, mogłaby pani marszałek teraz zarządzić przerwę, szybko zwołać Konwent Seniorów, o co wnioskuję, i położyć kres tej praktyce sejmowania na rympał, na wyścigi między północą a bliżej nieokreślonymi godzinami nadrannymi. Miejcie choć tyle przyzwoitości, choć forsujecie tutaj w tej sali czy właściwie teraz w przestrzeni wirtualnej, co tam chcecie, ale miejcie tę przyzwoitość, żeby dać nam przeczytać to, nad czym właściwie mamy tutaj głosować.

Konwentu nie zwołam, ale wniosek o przerwę jest regulaminowy, więc przegłosujemy wniosek o przerwę.

Wniosek został odrzucony. Przecież mam tablicę przed sobą. Proszę. Pani Marszałek! Wnoszę o odroczenie obrad do godz. Mienicie się partią, która walczy o prawa socjalne, ale zgromadzone tu osoby pracują wbrew Kodeksowi pracy. Czy nie potraficie zorganizować prostej pracy Sejmu? To, że pan, panie prezesie, nie cierpi parlamentaryzmu, ja rozumiem, ale nie sprowadzajmy polskiego Sejmu do atrapy, nie naruszajmy praw pracowniczych. Nie pokazujcie wszystkim, gdzie ich macie. Szanujcie elementarne zasady. Ale nie, wy udajecie, robicie wielki pic. Chcecie udawać, jak to ciężko pracujecie, a jutro będziecie na nowo łatać tę tarczę?

Po drugie, panie pośle, pan pierwszy deklarował pracę, ciężką pracę, i taką pracę prowadzimy.

W związku z tym, ponieważ padł wniosek formalny o odroczenie posiedzenia, poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek odrzucił. Właściwa komisja przedłożyła sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Sprawozdanie to druk nr 341. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 13. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druki nr 340 i 341) Proszę pana posła Henryka Kowalczyka o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła uchwałę Senatu skierowaną przez panią marszałek do Komisji Finansów Publicznych, uchwałę Senatu dotyczącą ustawy sejmowej o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Komisja w dniu dzisiejszym rozpatrzyła wszystkie poprawki i rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie 45 poprawek spośród tych, które zaproponował Senat, a 50 poprawek proponuje odrzucić.

Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Wniosek formalny. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Sytuacja jest nadzwyczajna. Polska czeka na nasze decyzje. Kancelaria Sejmu musi przygotować odpowiednie dokumenty, żeby trafiły na biurko pana prezydenta, tutaj liczy się każdy dzień. Wobec tego składam wniosek o głosowanie wspólne: nad poprawkami, które rekomenduje komisja, oraz nad poprawkami, których komisja nie rekomenduje. Słyszę, że jest głos przeciw. Pan poseł Borys Budka. Bardzo proszę. Oczywiście jestem przeciwny temu wnioskowi. Nawet nie będziecie wiedzieli, nad czym głosujecie. Co więcej, szanowni państwo, w tej chwili drugi raz odrzucicie poprawkę gwarantującą dużo więcej testów, w tym testy dla wszystkich pracowników służb medycznych, tzn. właśnie chcecie to zrobić. Wsłuchajcie się w głos waszych kolegów, np. pana Sośnierza, który mówi wyraźnie: Chcecie odmrażać gospodarkę? To trzeba przeprowadzać kilkadziesiąt tysięcy testów dziennie. Wy zaraz odrzucicie pieniądze, które są na to przeznaczone. Zastanówcie się, kochani, czy wy chcecie prawdziwej zmiany, prawdziwego ratowania gospodarki, czy wy po raz kolejny robicie tak jak pan premier od wielu, wielu miesięcy - tylko powerpointowy pic.

Każda poprawka warta jest przyjęcia. Gwarantuję.

Usłyszałam sprzeciw. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem propozycji głosowania łącznego nad poprawkami Senatu zgodnie z przedstawioną przeze mnie propozycją, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm propozycję przyjął.

Panie pośle, jesteśmy w trakcie głosowania. Jesteśmy w trakcie głosowania, panie pośle, proszę usiąść. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem ww. poprawek, zechce nacisnąć przycisk.

Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem ww. poprawek, zechce nacisnąć przycisk.

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Informacja o wpływie interpelacji, zapytań oraz odpowiedzi na nie dostępna jest w Systemie Informacyjnym Sejmu. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu. Informacja o terminie i porządku dziennym 11. posiedzenia Sejmu zostanie paniom i panom posłom doręczona.